Wysoka Izbo! Zwracam się z wnioskiem formalnym o odroczenie obrad do wtorku, żeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej mógł opublikować ustawę, która daje dodatki dla medyków i dla personelu medycznego. Do dzisiaj ta ustawa nie została opublikowana, tymczasem dzisiaj ma zostać w Wysokim Sejmie przeforsowana ustawa, która dodatki dla medyków zabiera. I trzeba powiedzieć jasno, że to jest pierwszy na świecie, pierwszy w historii rząd w demokratycznym kraju, który w szczycie epidemii chce zabrać dodatki dla lekarzy i dla personelu medycznego. To jest absolutny skandal i my się na to absolutnie nie godzimy. Jednocześnie w tym samym czasie Wysoki Sejm pod wodzą PiS-u chce nałożyć na Polaków nowe podatki, na ponad 40 tys. spółek komandytowych. I tu cytat z pana premiera Morawieckiego: Nowe podatki są potrzebne po to, by ratować polskich przedsiębiorców. Przecież to jest logika, która nie ma w sobie nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Niszczycie polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj ledwo żyją, przez wasze niespójne prawo, przez regulacje, które wprowadzacie, i przez chaos prawny, który wprowadziliście. Dziękuję bardzo. Padł wniosek o odroczenie posiedzenia, ale jeszcze dwa wnioski formalne. Wysoka Izbo! Dokładnie 28 listopada 1918 r., 102 lata temu, Polki uzyskały prawa wyborcze. To wielka rocznica dająca odpowiedzialność za nasz kraj dziewczynom, kobietom, naszym przyjaciółkom, koleżankom, które budowały odpowiedzialność taką, jak mężczyźni. Dzisiaj taka sama odpowiedzialność spoczywa na wnuczkach i prawnuczkach, które protestują na ulicach polskich miast, walcząc o swoje prawa. Prawo do głosowania to prawo do decydowania. I mówię to jako mężczyzna, bo uważam, że nie może być podziału na mężczyzn i kobiety, którzy mają różne prawa.

Oczywiście to nie był wniosek formalny. Proszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu poddania jednak pod głosowanie uchwały, którą wczoraj przedłożyliśmy pani marszałek, pod którą podpisali się posłowie Konfederacji i Solidarnej Polski. To uchwała, która odpowiada na urojenia Parlamentu Europejskiego, któremu wydaje się, że może recenzować prace najwyższych polskich władz w sprawach zastrzeżonych do ich wyłącznych kompetencji.

Wczorajszy precedens staje się powoli zwyczajem. Nie możemy pozwalać na to, żeby w sprawach, które należą do polskich kompetencji, Parlament Europejski się wypowiadał. My nie recenzujemy pracy innych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego i oczekujemy w tym względzie wzajemności. Dziękuję, panie pośle.

Sejm wniosek odrzucił. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Działa, już działa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 787 i 788. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Senat podjął uchwałę odrzucającą ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, druk nr 786. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej uchwały. Proponuję, na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu, rozpatrzenie uchwały bez uprzedniego skierowania jej do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Planowany punkt 62. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 783 i 787) Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu omówiła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 783. Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 poprawki, pozostałe poprawki zostały zaopiniowane negatywnie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy.

Nikt nie był za, 446 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 24. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

10 - za, 437 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

1 - za, przeciw - 449, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 784 i 788) Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie przedmiotowej ustawy. Senat zaproponował 30 poprawek. Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie 14 poprawek i rekomenduje ich przyjęcie. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawki od 1. do 9. zostały zgłoszone do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Nikt nie był za, 451 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Z poprawką tą łączy się 16. poprawka Senatu. Głosujemy.

2 - za, 450 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 8. i 17., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, przeciw - 455, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 27. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 40. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 786) Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą.

Wysoka Izbo!

Możecie się panowie posłowie uspokoić? Jak nie chcecie, możecie wyjść. Panie pośle! Pan poseł wygłasza oświadczenie. Jak zawsze - nie macie kultury. Nie bez znaczenia dla wybuchu powstania były ruchy rewolucyjne płynące z Europy. Początkiem zrywu był spisek w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie kierowany przez por. Piotra Wysockiego. Młodzi podchorążowie oraz studenci, a więc i cywile, i wojskowi, stanęli ramię w ramię, atakując Belweder, siedzibę księcia Pawłowicza - brata cara Mikołaja I. 18 grudnia pod presją opinii społecznej i rozbudzonego ducha walki o niepodległość Sejm uznał powstanie za narodowe. Ważnym elementem było kontruderzenie gen. Ignacego Prądzyńskiego. Niestety nieskuteczne ataki gen. Jana Skrzyneckiego przerwały początkowe zwycięstwa Polaków. Powoli spadało morale wojska polskiego. W lipcu po szturmie na Warszawę, obronie Woli i śmierci gen. Sowińskiego nastąpiła kapitulacja. Skutkiem powstania były pacyfikacja i militaryzacja Królestwa Polskiego, ostre represje Rosjan, ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, zastąpienie konstytucji statutem organicznym, zniesienie Sejmu i samorządów oraz całkowita rusyfikacja. Zbudowano cytadelę, zrujnowano polskie szkolnictwo, a powstańców wcielono do armii rosyjskiej lub zesłano w głąb Rosji. Warto przypomnieć, że powstańcy nie doczekali się pomocy z zewnątrz, nawet ze strony dyplomacji państw zachodnich. Powstanie na pewien czas zachwiało potęgą Rosji. Nie zakończyło się kapitulacją czy układami, lecz właśnie emigracją. Książę Adam Czartoryski stwierdził, iż opór, jaki rewolucja polska stawiła siłom Cesarstwa Rosyjskiego, zadziwił Europę, jak również nagły jej upadek. Być może Europa nie dziwiłaby się tak bardzo, gdyby choć trochę pomogła polskim powstańcom. Wysiłek powstania nie poszedł na marne. Wskrzeszono walkę o niepodległość i udowodniono, że sprawa polska to nie jest coś, co można załatwić połowicznie, jak chociażby na kongresie wiedeńskim. Naród polski zaszczepił w sobie wartości patriotyczne i pokazał, że chce przywrócenia kraju w jego pierwotnych granicach. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska.

Wysoki Sejmie! Moje oświadczenie dotyczy drastycznych ograniczeń dla branży turystycznej w czasie nadchodzącej zimy. Z turystyki żyje 80% mieszkańców gmin górskich i podgórskich, a więc znacząca część naszego społeczeństwa. Samorządy i przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne turystów i mieszkańców i jednocześnie nie burzyć wszystkiego, co funkcjonuje dookoła, nie doprowadzać do ogólnego bankructwa całej branży turystycznej, któremu nie są w stanie zapobiec niewspółmiernie niskie i wybiórcze rekompensaty planowane przez rząd. Dlaczego więc wicepremier Gowin i podległe mu ministerstwa nie podjęli dialogu z przedsiębiorcami i samorządami gmin górskich przed podjęciem tak drastycznych ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej? To wprost niewiarygodne, jak przedmiotowo traktuje się prawdziwych i odpowiedzialnych gospodarzy górskich kurortów. Samorządy gmin górskich wystąpiły do premiera Gowina z konkretnymi propozycjami rozwiązań, których zastosowanie wyeliminowałoby rozprzestrzenianie się zachorowań, koronawirusa. Górskie kurorty od lat, budując infrastrukturę turystyczną, zawsze dbały o możliwie najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do wypoczynku. W ich ocenie miejscowości górskie są najlepiej przygotowane do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. W bieżącym roku, w okresie letnim i jesiennym, miejscowości te gościły kilka milionów turystów, mimo to zachorowalność mieszkańców i turystów była znikoma. Wpływ na to mają takie czynniki, jak położenie geograficzne i właściwa organizacja przestrzeni publicznej. W ostatnich dniach samorządy w porozumieniu z przedsiębiorcami przedstawiły rządowi szereg konkretnych rozwiązań dotyczących branży hotelowej, gastronomicznej, stref rekreacji i wypoczynku, które są gotowe natychmiast wdrażać. Obecnie oczekują na pilną odpowiedź. Gospodarze gmin zwracają uwagę na bezwzględną konieczność traktowania branży turystycznej jako całości, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów działalności, a więc: nocleg, gastronomia, wypoczynek, rekreacja. Chodzi o zorganizowanie ferii zimowych przez 10 tygodni w celu rozłożenia natężenia ruchu turystycznego, zapobieganie odpływowi turystów poza granice naszego kraju, traktowanie rekompensat jako ostatecznego rozwiązania, gdyż większość ludzi rekompensat nie otrzyma.

Apeluję do pana premiera o pilne rozpatrzenie złożonych propozycji i podjęcie rozmów z wiarygodnymi i równorzędnymi partnerami, jakimi są przedsiębiorcy i samorządowcy gmin górskich. I bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejszy dzień to czarny dzień dla polskiej służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość zabrało należne dodatki, które należą się lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, technikom RTG, pracownikom sterylizacji, salowym, pracownikom kuchni i pracownikom technicznym pracującym w szpitalach, które walczą o życie i zdrowie Polaków, w szpitalach, które walczą z COVID-em. Jest takie polskie przysłowie: kto daje i odbiera. Moi wyborcy bardzo by chcieli wiedzieć i poznać personalnie, z imienia i nazwiska osoby, które przygotowały w Polsce plan sabotowania służby zdrowia oraz systematycznego niszczenia zasobów ludzkich odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej służby zdrowia. W 2005 r. Polska przyjęła dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie zasad kształcenia pielęgniarek, stawiając im bezwzględny wymóg ukończenia studiów wyższych. Kierowano się wtedy dobrem pacjenta. Nie pomyślano jednak, aby w ślad za zwiększonymi wymaganiami odpowiednio zwiększyć uposażenie kadry medycznej średniego szczebla, co doprowadziło do emigracji pielęgniarek i uzasadnionych protestów całego środowiska. W bieżącym roku rząd w odpowiedzi na niezadowolenie kadry pielęgniarskiej, pomimo że ogłosił jej olbrzymi niedobór na rynku pracy, zatrudnił jedynie ok. 1 tys. z łącznej liczby ponad 4 tys. osób, które ukończyły studia pielęgniarskie. Pozostałe 3 tys. osób, które odbyły bardzo kosztowne studia, zasiliły zachodnie rynki pracy albo musiały się przekwalifikować. Te sam rząd jednocześnie forsuje w Sejmie ustawę, która na polski rynek pracy dopuszcza pielęgniarki po szkole średniej i z bardzo wątpliwą znajomością języka polskiego. Tym oto sposobem PiS wydaje publiczne pieniądze podatników na studia wyższe dla kadry medycznej średniego szczebla, którą następnie zmusza do emigracji. Polska kształci pielęgniarki dla Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Do opieki nad polskimi pacjentami natomiast będzie się ściągać pielęgniarki bez wyższego wykształcenia, gotowe pracować za połowę stawki, które swoje wykształcenie zdobyły w przyszpitalnych szkołach średnich w Uzbekistanie, Iranie czy Etiopii. Jedynym wymogiem formalnym pozwalającym na podjęcie pracy jest pisemne oświadczenie o znajomości języka polskiego, przy czym ustawa nie określa, czy oświadczenie to musi być napisane w naszym narodowym języku. Działania takie w żadnym wypadku nie mogą być przypadkowe i noszą wyraźnie znamiona działalności na szkodę polskiej służby zdrowia oraz pacjenta. Sprawę powinny gruntownie zbadać służby specjalne zarówno pod kątem korupcyjnym, jak i kątem działalności na szkodę Skarbu Państwa. Natomiast nasze służby specjalne - po blamażu związanym z rozpoznaniem dostaw nieistniejących respiratorów oraz niezdolnością do odzyskania milionów od handlarza bronią - zostały najwyraźniej wyposażone w metalowe pałki i skierowane do bicia demonstrujących kobiet, więc raczej nie znajdą czasu na zajęcie się tą sprawą. Dzisiejszy dzień to czarny dzień dla polskiej służby zdrowia. I bardzo proszę, pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałbym zwrócić uwagę w tym punkcie na problem, z którym borykają się już od wielu lat mieszkańcy Zabrza. Chodzi mi o pokopalniane zwałowisko Ruda w dzielnicy Biskupice, które to od lat zatruwa życie - dosłownie i w przenośni - mieszkańcom najbliżej położonych dzielnic. Biskupicka hałda, pozostałość po nieistniejącej już kopalni Zabrze, zajmuje powierzchnię ponad 27 ha. Zdeponowano na niej prawie 2 mln t odpadów stanowiących zagrożenie samoczynnym zapłonem lub ingerencją zewnętrzną. Najgorzej jest oczywiście latem, gdy żar leje się z nieba. Nie sposób wtedy w pobliskich mieszkaniach otworzyć okien, ale i o każdej porze roku skutki są bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Niestety podjęte wtedy prace nie dały pożądanego rezultatu. Część zabrzan wręcz twierdzi, że działania te spowodowały zapłon kolejnej partii składowiska. Problem dymiącej hałdy wielokrotnie był omawiany podczas sesji rady miasta czy też szeroko opisywany w lokalnych mediach. Niestety nie został rozwiązany do dziś. W spotkaniu, które miało charakter wizji lokalnej, oprócz radnych udział wzięli naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Zabrze oraz ekspert z Głównego Instytutu Górnictwa prowadzącego badania na czynnej hałdzie Ruda. Komisja omawiała kilka wariantów rozwiązania tego problemu, w tym także rozbiórkę hałd. Na koniec ustalono, że najrozsądniejszym i zarazem bezpiecznym rozwiązaniem będzie systematyczne gaszenie hałdy oraz wprowadzenie rozwiązań zapobiegawczych. Działania te wiążą się jednak z dodatkowymi, niemałymi środkami finansowymi. Zabrze o aplikowanie do wojewody śląskiego o przyznanie dodatkowych środków potrzebnych do rekultywacji hałdy. Panie Premierze! Śląsk jest regionem, w którym zanieczyszczenie powietrza jest największe w naszym kraju. Dlatego apeluję do pana z tego miejsca o wsparcie i pomoc, aby problem związany z hałdą Ruda w Zabrzu został dla zdrowia mieszkańców mojego miasta jak najszybciej rozwiązany. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym zakończyliśmy 21. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny kolejnego posiedzenia Sejmu zostanie panom i paniom posłom doręczony.